Szanowni Państwo! Zmiana 1. odnosi się do art. 5 Kodeksu wyborczego i jest ściśle powiązana ze zmianą 19., która odnosi się do art. 181 Kodeksu wyborczego. Pragnę podkreślić, że obwodową komisję wyborczą do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodach i obwodową komisję wyborczą do spraw ustalenia wyników głosowania powołuje się tylko w ogólnokrajowych wyborach samorządowych. To oznacza, że w pozostałych wyborach pozostawiamy tylko jedną komisję. Wybory samorządowe są na tyle skomplikowane i wymagają tak obszernej pracy, że uzasadnione jest powołanie dwóch komisji: jednej do przeprowadzenia głosowania, drugiej zaś do ustalenia wyników. Kolejna zmiana odnosi się do art. 11 zawartego w rozdziale 2, który to rozdział reguluje prawa wyborcze. W tym artykule proponujemy nowy zapis, tak aby ujednolicić przepisy Kodeksu wyborczego z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych poprzez uregulowanie w Kodeksie wyborczym kwestii biernego prawa wyborczego w sposób podobny do uregulowania tej sprawy w przepisach dotyczących pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyborów lub powołania.

Przyjęcie tej poprawki zlikwiduje istniejącą kolizję prawną pomiędzy obiema ustawami. Jest to postulat również Państwowej Komisji Wyborczej. Pragnę zasygnalizować, że w obecnym stanie prawnym decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Projekt zakłada wydłużenie terminu na rozpatrzenie wniosku i wydanie rozstrzygnięcia o prawie wpisania lub odmowie wpisania do rejestru wyborców do 5 dni. Jest to wniosek samorządowców. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci wskazywali, że weryfikacja w okresie 3 dni jest terminem zbyt krótkim. Szanowni Państwo!

Tutaj dokonujemy usunięcia kolizji pomiędzy trzema artykułami Kodeksu wyborczego. Zapisy wprowadzają możliwość obiegowego podejmowania uchwał przez Państwową Komisję Wyborczą w sprawach niecierpiących zwłoki, gdy nie ma możliwości zwołania posiedzenia komisji. Warto zaznaczyć, że niektóre zadania są obarczone krótkim terminem, np. 2–3 dni, to jest zbyt mało do podjęcia takiej uchwały, dlatego też projekt ustawy wprowadza tego typu rozwiązanie i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Państwowej Komisji Wyborczej i usprawnia proces wyborczy. Kolejna istotna zmiana pojawia się w art. 170. W obowiązującym stanie prawnym komisarze nie muszą być sędziami. Proponuje się zmianę przepisów w taki sposób, aby w skład okręgowych komisji wyborczych wchodziło od czterech do 10 sędziów i z urzędu, jako jej przewodniczący, komisarz wyborczy, natomiast w rejonowej komisji wyborczej - czterech sędziów i z urzędu, jako jej przewodniczący, komisarz wyborczy. Pragnę podkreślić, że komisarz wyborczy w chwili obecnej nie musi być sędzią i tutaj też likwidujemy pewną nieścisłość. Warto przytoczyć zmiany, jakie dotyczą art. 182. W tej zmianie pragniemy zróżnicować składy komisji wyborczych i te składy będą uwarunkowane ilością mieszkańców w obwodzie. Pozostałe zapisy art. 182 szczegółowo opisują, szanowni państwo, mechanizm powołania członków do obwodowej komisji wyborczej spośród osób zgłoszonych przez komitety wyborcze, a w przypadku gdy komitety nie skorzystają z przysługujących praw, zgłoszenie kandydatów pozostawia się komisarzowi wyborczemu, który uzupełnia komisję do pełnego składu spośród wyborców spełniających warunek w § 4, choćby ukończony 18. rok życia.

Kolejną zmianą w tym artykule jest to, iż kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat na dzień zgłaszania do komisji, a nie na dzień wyborów, jak to było do tej pory. Wydaje się to bardzo rozsądne, dlatego że taka osoba potem wykonuje wiele czynności prawnych, a jeszcze nie jest tak naprawdę osobą pełnoletnią.

Wygląda to w ten sposób, że osoba spokrewniona z kandydatem w wyborach może być członkiem obwodowej komisji wyborczej właściwej dla innych okręgów wyborczych niż okręg, w którym kandyduje osoba z nią spokrewniona. Wydaje się, że do dzisiaj ten zapis był zbyt restrykcyjny. W tej chwili doprecyzowujemy, aby taka osoba mogła zasiadać i pracować w innych komisjach poza tą komisją, z której kandyduje osoba spokrewniona.

Wskazujemy te przypadki: nieuczestniczenie w pracach bez usprawiedliwienia lub podejmowanie działań sprzecznych z prawem. Komisarz ma plenipotencję, aby odwołać taką osobę. Szanowni Państwo! Warto zwrócić uwagę na kolejną zmianę, jaka się pojawia w art. 218, która wypełnia postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, a właściwie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2012 r., który to trybunał uznał, że część przepisu art. 218 ust. 2 dotycząca braku środka odwoławczego w tym zakresie jest niezgodna z konstytucją. Dlatego dokonujemy zmiany, iż od postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej przysługuje skarga do Sądu Najwyższego w terminie 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez PKW, a Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w ciągu 2 dni w składzie trzech sędziów w postępowaniu nieprocesowym. Szanowni Państwo! Pojawiają się zmiany w trybie odwoławczym i one odnoszą się zarówno do art. 300, art. 304, art. 404 czy też art. 405.

Państwowa Komisja Wyborcza zwracała nam uwagę na to, że bardzo często organy wyborcze miały trudność z dotarciem do pełnomocników wyborczych, nie odbierano telefonów. Pragnę podkreślić, że Państwowa Komisja Wyborcza to nie jest instytucja detektywistyczna czy też Polski Czerwony Krzyż, żeby poszukiwać ludzi, tylko jest po to, żeby w tym bardzo intensywnym czasie wykonywać swoją pracę. W związku z tym właśnie taka zmiana pojawia się w tych czterech artykułach. Kończąc swoje wystąpienie, pragnę podkreślić, że według projektu ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z uwagi na ważny interes państwa, zaś zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie, aby ta ustawa została przyjęta. Projekt wywołuje pozytywne skutki społeczno-gospodarcze choćby poprzez to, że pojawia się jedna komisja, a nie tak jak do tej pory w przepisach - dwie przy wszystkich wyborach. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Dziękuję, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Głos ma pani poseł Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy. Szanowni Państwo! 11 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa wprowadziła liczne zmiany w zakresie prawa wyborczego, w szczególności zaś odnoszące się do wyborów do jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotowy projekt zawiera szereg uregulowań, które mają za zadanie przyczynić się do dostosowania zmian wprowadzonych w styczniu 2018 r. do wszystkich rodzajów wyborów oraz mają na celu usprawnienie procedury wyborczej. Bardzo ważną zmianą zawartą w projekcie, będącą niejako ukłonem w kierunku obywateli, jest wprowadzenie możliwości dokonywania zgłoszeń do składów obwodowych komisji bezpośrednio przez wyborców, a nie jedynie przez komitety wyborcze. Ponadto proponuje również ważną zmianę dotyczącą przepisów w zakresie powoływania obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z nią w każdym obwodzie głosowania miałoby się powoływać obwodową komisję wyborczą w wyborach do Sejmu i Senatu, w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w toku kadencji, a także w wyborach uzupełniających do Senatu, oraz obwodową komisję wyborczą do spraw przeprowadzania głosowania w obwodzie i obwodową komisję wyborczą do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w związku z zakończeniem kadencji. Istotną zmianą zawartą w projekcie jest również pozbawienie biernego prawa wyborczego osób skazanych za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego bądź przestępstwo karnoskarbowe na jakąkolwiek karę. Dotychczas możliwości kandydowania pozbawione były bowiem tylko osoby skazane na karę pozbawienia wolności. Należy zauważyć, że projekt nie wywołuje dodatkowych kosztów finansowych dla budżetów jednostek samorządów terytorialnych. Wręcz przeciwnie: zmiana przepisów w zakresie powoływania dwóch komisji obwodowych tylko w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w związku z zakończeniem kadencji rad przyczyni się do zaoszczędzenia w budżecie państwa kosztów przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów. Nie ulega również wątpliwości, że jego wprowadzenie przyniesie pozytywne skutki społeczne np. w zakresie zwiększenia dostępności pewnych działań czy funkcji. W związku z powyższym Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera przedmiotowy projekt. Pan poseł Mariusz Witczak, Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Prawo i Sprawiedliwość zawsze traktowało ordynację jako przeszkodę stojącą na przeszkodzie do utrwalania władzy, do zdobycia pełni władzy.

Tym razem proponujecie rozwiązania, które mają charakter niekonstytucyjny, bowiem dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego bardzo wyraźnie mówią o tym, że należy zachować ciszę legislacyjną na 6 miesięcy przed pierwszą czynnością wyborczą. Zmieniacie kilka przepisów w rozdziale, który dotyczy również wyborów do Parlamentu Europejskiego, zatem łamiecie już to orzeczenie Trybunału.

Manipulowaliście kodeksem przy wyborach samorządowych, przy wyborach do Parlamentu Europejskiego, a teraz chcecie manipulować przy przepisach dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Bardzo gorąco chcemy Wysoką Izbę zachęcać do tego, żeby przestrzegać konstytucji i orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo proszę, pan poseł Jacek Protas, Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Szanowni Państwo! To, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło z Kodeksem wyborczym rok temu, woła o pomstę do nieba - niekompetencja, nieudolność, oczywiście działanie niekonstytucyjne.

Doprowadziliście do chaosu w czasie wyborów. Nie można było powołać urzędników wyborczych na czas. Nie można było zwołać pełnego składu komisji wyborczych. Liczenie głosów często trwało nie wiele godzin, ale wręcz wiele dni. Dzisiaj, gdybym był naiwnym młodzieńcem, a nie posiwiałym, dojrzałym człowiekiem, pewnie bym sobie pomyślał, że może chcecie naprawić te błędy, poszliście po rozum do głowy, chcecie naprawić to, co zepsuliście, i wprowadzacie szereg zmian dotyczących właśnie powoływania urzędników wyborczych, komisji itd., itd., po to ażeby proces wyborczy rzeczywiście przebiegał w sposób prawidłowy. Ale tak nie jest, bowiem to jest tylko zasłona do tego, ażeby przygotować polowanie z nagonką na niepokornych i niezależnych samorządowców. A teraz potrzebujecie amunicji dla odpowiednich służb i prokuratury, ażeby odstrzelić tychże niepokornych i samodzielnych wójtów, burmistrzów, prezydentów. Komunikat będzie otóż taki: Panie wójcie, panie prezydencie, jak będziecie niepokorni, jak nie będziecie realizować polityki zgodnie z naszym oczekiwaniem, to coś na was znajdziemy. Chociażby nawet przestępstwo, w przypadku którego sąd uzna kogoś winnym, a nawet nie wymierzy kary - nawet wtedy w wielu przypadkach taka osoba nie będzie mogła kandydować w zbliżających się wyborach. Poza tym budujecie podwójne standardy. Mówicie, że nie, ale tak jest. Dlaczegóż nie będzie mógł startować w taki sposób ukarany wójt, burmistrz, prezydent, a wszyscy inni będą mogli - na radnych czy też do Sejmu, Senatu, na prezydenta Rzeczypospolitej? To są podwójne standardy. Dlatego też, szanowni państwo, klub Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska nie zgadza się z takim sposobem procedowania, niekonstytucyjnym, [[Dzwonek]] i nie zgadza się z takimi zmianami. Dziękuję. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw propozycjom i uwagom Państwowej Komisji Wyborczej.

Poza tym przypominamy, że trzeba wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze, [[Oklaski]] po to by obywatele mieli możliwość odwołania swoich przedstawicieli, którzy nie dotrzymują swoich obietnic. Dziękuję bardzo. Pan poseł Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe - Unia Europejskich Demokratów. Wysoka Izbo! Rozpoczynamy dzisiaj. czwartą część maratonu, który można określić mianem bitwy władzy o Kodeks wyborczy. Za niecałe 4 miesiące bowiem czekają nas wszystkich wybory do Parlamentu Europejskiego, więc Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło kolejną turę majstrowania przy przepisach Kodeksu wyborczego. Obecna kadencja Sejmu obfituje w ustawy specjalne. Mieliśmy lex Szyszko, lex deweloper, mieliśmy próbę poszerzenia granic Warszawy o ościenne powiaty. Teraz mamy, można powiedzieć, lex Zdanowska, projekt oczywiście poselski z podpisami polityków PiS. W czasie kampanii w województwie łódzkim, a szczególnie w Łodzi, nieustanny partyjny przekaz o wygaszaniu mandatu jeszcze niewybranego, a już odwołanego prezydenta był wszechobecny. Łodzianie zdecydowali jednak inaczej. Dostrzegli fałsz i obłudę, a swój sprzeciw wyraźnie pokazali przy urnie wyborczej, udzielając ponad 70-procentowego poparcia pani prezydent. Przechodząc do szczegółów projektu - zmienione mają zostać przesłanki warunkujące możliwości kandydowania w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta. Nowelizacja ma pozbawić biernego prawa wyborczego w sytuacji skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Bardziej precyzyjnie - gdy osoba zostanie skazana na karę grzywny, nie będzie mogła kandydować. Mamy więc sytuację, że wielki przestępca, który musi zapłacić grzywnę w wysokości 500 zł, traci możliwość weryfikacji w wyborach i poddania się osądowi społecznemu. Co ciekawe, przepis ten ma dotyczyć tylko kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów.

Wprowadza się także nierównowagę między wójtem a lokalnym radnym, bo dzisiaj radnym może być osoba skazana, o ile nie jest to kara pozbawienia wolności. To pytanie już teraz kieruję do pani poseł przedstawiającej ten projekt. Widać, że duch małego Kazia nadal towarzyszy radosnej twórczości wnioskodawców, którzy tworzą te w istocie podwójne standardy.

W końcu z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że istotne zmiany w prawie wyborczym nie powinny być dokonywane w okresie co najmniej 6 miesięcy przed zarządzeniem wyborów. Tu także widać, że prawo macie za nic.

Dziękuję. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Poselskiego Nowoczesna przedstawiam stanowisko w kwestii poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, druk nr 3163.

zmianami istotnymi.

To jest skandaliczny sposób tworzenia prawa. Chcecie państwo wprowadzić obwodowe komisje wyborcze bez komisji do liczenia głosów we wszystkich wyborach poza wyborami samorządowymi. Naprawdę ani przesłanki z państwa uzasadnienia projektu, ani też żadne racjonalne przesłanki nie przemawiają za różnicowaniem tych różnych wyborów.

Państwo tego niestety nie robicie. Traktujecie prawo wyborcze bardzo instrumentalnie, stricte politycznie. Dziękuję. Wysoka Izbo! Stanowisko Koła Poselskiego Wolni i Solidarni odnośnie do przedstawionego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy jest pozytywne, jednakże żeby zoptymalizować te dobre zapisy, pozwolimy sobie zgłosić podczas posiedzenia komisji stosowną poprawkę. Dziękuję.

Wysoka Izbo! Można byłoby zadać pytanie, po co i dlaczego znowu są teraz kolejne zmiany. Są dwie sprawy dyskusyjne, o których mówili poprzednio moi koledzy, ale ja to powtórzę. Pierwsza sprawa to powrót do powoływania jednej obwodowej komisji wyborczej. Pytanie: Po co państwo robili wcześniej taki myk, żeby były te dwie komisje, żeby w jednej komisji było to liczone, a w drugiej żeby głosować? Wtedy państwo mówiliście, że robicie to po to, aby zapewnić bezpieczeństwo i uczciwość. Może po prostu wystarczyłoby, ogłaszając dzisiaj ten projekt, powiedzieć, że przyznajecie się do błędu i wracacie do tego, co było. To jest jedna rzecz.

Nie może kandydować osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, podczas gdy we wszystkich innych wyborach nie może kandydować osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. I na pierwszy rzut oka można byłoby powiedzieć i wydawać by się mogło, że czemu mamy pozwalać skazanym na kandydowanie w wyborach, prawda? W zasadzie wszyscy powinniśmy się zgodzić, tylko że to prawo nie dotyczy ani posłów, ani senatorów, ani radnych i wybieranych z ich grona starostów powiatowych i marszałków województwa. Wprowadzacie państwo w tym artykule zasadę, że są równi i równiejsi. I to jest jeden z najgłupszych pomysłów, jakie państwo przedstawiacie, jeżeli chodzi o Kodeks wyborczy i wszystkie pomysły, które wprowadzaliście przez ostatnie 2 lata. My będziemy za odrzuceniem tego projektu. Dziękuję. Jeśli ktoś z państwa chce się zapisać do głosu, zapraszam. Zamknę listę po pierwszym pytaniu. Czas pytania - 1 minuta. Głos ma pan poseł Michał Szczerba. Czy jest pan poseł? Jest pan poseł. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Można powiedzieć: a nie mówiliśmy, ponieważ ten projekt zakłada powrót do jednej obwodowej komisji wyborczej, ale cały czas z niezrozumiałych dla nas względów, z wyjątkiem wyborów samorządowych, najbardziej skomplikowanych, bo przecież o wiele bardziej skomplikowanych organizacyjnie niż wybory do Parlamentu Europejskiego, Sejmu, Senatu czy też na prezydenta. Chciałbym bardzo powiedzieć, że ta sytuacja z dwoma komisjami obwodowymi spowodowała dużo zamieszania. Spowodowała również - to jest wynik obserwacji - że nawet w dużych miastach te komisje pracowały bardzo często w minimalnym dopuszczalnym prawnie składzie pięciu osób, a niedobór członków skutkował m.in. długimi kolejkami do urny. Pytanie jest następujące: Dlaczego projektodawcy nie wracają do kwestii definicji znaku X? Czy to nie jest dobry moment, żeby wrócić do poprzedniej definicji, która była dla wszystkich zrozumiała? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję. Wysoka Izbo! Ale gdy wprowadzano zmiany, właśnie w poprzednim roku, to wynikały one z braku wyobraźni, bo Kodeks wyborczy jest specyficzną ustawą, ustawą o bardzo dużej staranności legislacyjnej.

Dwa.

Uregulowanie elementów prekampanii.

Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Artur Dunin. Czy jest pan poseł Dunin?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tu już padły słowa z tej mównicy. Państwo znowu łamiecie konstytucję tą ustawą.

To jest ponad 250 tys. głosów. Dzisiaj ta ustawa daje wam możliwość zniweczenia tych szans, wysiłku łodzian. Pani poseł Małgorzata Niemczyk. Wysoka Izbo! Nie mogliście z samorządowcami wygrać w jesiennych wyborach w uczciwej walce, więc co dzisiaj robi Prawo i Sprawiedliwość? Zmienia Kodeks wyborczy, aby pokonać panią prezydent Hannę Zdanowską i pokonać łodzian.

Nie potraficie jej pokonać w wyborach. Boicie się jej, boicie się zaufania, którym łodzianie ją obdarzają. W projektowanych zmianach nie uwzględniacie funkcji radnych, posłów, senatorów. Jeśli ta zmiana wejdzie w życie w obecnym kształcie, to można będzie być prezydentem Polski. Pytam: Czy Hanna Zdanowska będzie mogła sprawować swój urząd do końca kadencji, czy odwołacie ją wedle tej nowelizacji? Czy również będziecie zmieniać Kodeks karny? Dziękuję. Wysoka Izbo! Szef PKW wyraził zadowolenie z przedłożonego projektu ustawy, stwierdził jednak, że uwzględniono za mało postulatów zgłoszonych przez PKW. Moje pytanie do wnioskodawców: Czy zamierzacie pochylić się państwo nad postulatami zgłoszonymi przez PKW, które w tej ustawie nie zostały uwzględnione? Pan poseł Marek Wójcik. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W 2009 r. zmieniliśmy konstytucję w taki sposób, aby można było wprowadzić zakaz kandydowania osób skazanych do Sejmu, a dopiero w 2010 r. w Kodeksie wyborczym wprowadziliśmy przepisy, które były jednolite w odniesieniu i do posłów, i do samorządowców. Zrobiliśmy to w pełni świadomie, zrobiliśmy to przy pełnej akceptacji tej Sali. Przypomnę, że Kodeks wyborczy w 2010 r. został uchwalony jednomyślnie. To jest bardzo zły standard legislacyjny, jeżeli tak można powiedzieć. Ale o waszym standardzie legislacyjnym świadczy również fakt, że tę ustawę chcecie przyjąć dzisiaj, w ciągu jednego dnia. Chciałbym również spytać panią poseł, [[Dzwonek]] dlaczego wprowadzacie państwo przepis, który mówi o tym, że ta ustawa wchodzi w życie dzień po dniu ogłoszenia. Otóż zgodnie z polskim prawem standardowe jest 14-dniowe vacatio legis, a odejść od tej zasady można tylko z uzasadnionych powodów. Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Matusiewicz.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zmiany zaproponowane w projekcie poselskim absolutnie nie naruszają konstytucji.

Zapraszam. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Procedowana ustawa to bat na niepokornych prezydentów, burmistrzów, wójtów. Pod przykrywką nieznacznych zmian chcecie przygotować narzędzie dla służb i prokuratury w celu wyeliminowania niewygodnych samorządowców poprzez odebranie im biernego prawa wyborczego. Utratę tego prawa przewiduje się nawet w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przy czym chodzi tu o każdą karę, a nie tylko - jak dotychczas - o karę pozbawienia wolności. I to jest właśnie główny cel tej ustawy. Chciałabym jeszcze zapytać i zwrócić uwagę na to, aby organizacje pozarządowe mogły i miały taką możliwość zgłaszać do komisji swoich kandydatów. Pani poseł Zofia Czernow. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

Dlaczego stosujemy takie skróty przy tak ważnych ustawach? Po drugie, chciałam zapytać, czy wnioskodawcy posiadają opinie konstytucjonalistów na temat zgodności tych procedur z konstytucją. Dlaczego w tym wypadku wnioskodawcy nie zaopatrzyli nas w nią, a przynajmniej ja nie otrzymałam takiej opinii? I ostatnia sprawa - podwójne standardy w kwestii prawa wybieralności wójtów, burmistrzów i prezydentów. Dziękuję. Pani poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Wysoka Izbo! Znów powielam pytanie dotyczące przepisów o dodaniu tych zapisów o braku prawa wybieralności w wypadku osoby skazanej prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Proszę mi powiedzieć, czy przestępstwo w zakresie ruchu drogowego o niskiej szkodliwości i w efekcie skazanie prawomocnym wyrokiem na karę grzywny to będzie również przesłanka, by uniemożliwić kandydowanie na wójta, burmistrza i prezydenta. Bardzo proszę o konkretną odpowiedź. Dziękuję. Zapraszam pana posła Szymona Ziółkowskiego. Wysoka Izbo! Dlaczego wyższy standard moralności wedle projektu tej ustawy ma dotyczyć burmistrzów czy wójtów, a nie dotyczyć prezydenta naszego kraju? Dlaczego trudniej według tej ustawy będzie zostać wójtem czy burmistrzem, a nie prezydentem Rzeczypospolitej? Druga sprawa, która również wiąże się z tą ustawą, to oświadczenie o niekaralności. Dlaczego cały czas parlamentarzyści, kandydaci wybierani w wyborach muszą tylko i wyłącznie składać oświadczenia o niekaralności, a nauczyciel, trener czy sportowiec, który ubiega się o tzw. rentę olimpijską, muszą przedstawić zaświadczenie z sądu? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Piotr Pyzik. Nie ma pana posła? Jest.

Wysoka Izbo!

Chciałbym jednak zaapelować o nieustawanie w reformowaniu systemu przeprowadzania wyborów. Wciąż nierozwiązana pozostaje kwestia odpowiedzialności i weryfikowalności w zakresie tworzenia spisu wyborców, wciąż brakuje możliwości sprawowania powszechnej kontroli przez obywateli, choćby poprzez monitoring za pomocą kamery internetowej.

Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zmiany wprowadzone w Kodeksie wyborczym, czyli zakaz kandydowania do pełnienia funkcji burmistrza, prezydenta i wójta dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe na każdą karę jest dyskryminujący, ponieważ dotyczy tylko wójtów, burmistrzów i prezydentów. Nie dotyczy to też kandydatów na posłów i senatorów.

Także mam pytanie do pani, jeżeli chodzi o instytucję zatarcia. Jeżeli osoba była skazana, ukarana i wyrok uległ zatarciu, to czy taka osoba może kandydować, może startować? I dlaczego projekt jest niekonstytucyjny? Dlaczego pół roku przed wyborami wprowadzacie istotne zmiany w Kodeksie wyborczym? Bardzo proszę. Pani Marszałek! Tak się zastanawiałem właśnie, dlaczego te pytania są zadawane, dlaczego jest ta nowelizacja, która rzeczywiście wprowadza chaos, wprowadza te podwójne standardy.

Rzadko się zdarza, żeby projekty, które PiS przedstawia, służyły dobru wspólnemu, a jak służy dobru wspólnemu działalność PiS-u, pokazuje afera z taśmami Kaczyńskiego.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Przed wyborami samorządowymi zmieniliście Kodeks wyborczy. Wydawało wam się, że te zmiany pomogą wam wygrać. Niestety, nie udało się, przegraliście.

Mogłaby się ona odnieść do tych przepisów, które wprowadziliście kilka miesięcy temu, a które się nie sprawdziły. Wydaje się, że po prostu logika nakazywałaby wam to zrobić, tylko co zrobić, kiedy wam tej logiki brakuje? Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Trzeba mieć wyjątkowo dużo złej woli albo oczywiście nie znać ustawy, żeby twierdzić, że te zapisy, które proponujemy, mają zastosowanie do wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy obecnie pełnią funkcję właśnie wójta, burmistrza, prezydenta. Oczywiste jest, że bierne prawo wyborcze badane jest na moment kandydowania i zgłaszania kandydatur, zatem oczywiste jest, że ta okoliczność obecnych wójtów, prezydentów dotyczyć nie będzie. Szanowni Państwo! Jeżeli państwo z tej ustawy tego nie mogą wyczytać, to możliwe jest doprecyzowanie tych przepisów. Ale już dzisiejsze przepisy na to wskazują: na pewno do obecnych wójtów, prezydentów ta poprawka nie ma zastosowania. Dziękuję. Panie pośle. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pokrótce chciałabym powiedzieć, i uspokoić państwa, że ten projekt nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek standardów czy naruszenia konstytucji. Chcę zapewnić państwa i uspokoić - jeżeli państwo uważacie, że pani Zdanowska mogłaby dzięki wprowadzeniu tej ustawy utracić stanowisko prezydenta, to jestem gotowa wnieść taką poprawkę, która absolutnie uspokoi zarówno państwa, jak i panią prezydent. Nie to ma na celu ten projekt, ta nowelizacja. Wsłuchujemy się w głos Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego i chcemy po prostu usprawnić wybory. To dlatego powstał ten projekt. Po drugie, państwo mówicie, że różnicujemy, a jednocześnie składacie wniosek o odrzucenie tego projektu. Nie chcecie dyskutować na ten temat. Mówicie, że chcecie rozmawiać, a jednocześnie już tutaj zgłosiliście państwo wniosek o odrzucenie. Proszę państwa, nawet nie dajecie szansy rozmowy choćby w komisji, która zajęłaby się tym projektem.

Proszę zwrócić uwagę, że w odniesieniu do samorządowców są to wysokie wymagania, a w stosunku do osób, które nadzorują ich pracę, które odpowiadają za ich pracę, już te wymagania są zdecydowanie mniejsze. Jeszcze pragnę przypomnieć, że w ustawodawstwie polskim w odniesieniu do takich zawodów jak policjant, sędzia, detektyw, komornik, nauczyciel, prokurator, pracownik ochrony, pracownik kontroli skarbowej, notariusz, pilot wycieczek, agent ubezpieczeniowy, pracownik samorządowy stawiane są wymagania odnośnie do niekaralności. Tak że, proszę państwa, nawet jeśli twierdzicie, że w odniesieniu do władzy ustawodawczej powinien być ten sam wymóg, to może spróbujmy dyskutować w komisji, nie odrzucajmy już na wstępie projektu zaproponowanego na tym posiedzeniu przez nas, przez grupę posłów. Szanowni Państwo! Na szereg technicznych pytań państwo dostaniecie odpowiedź bezpośrednio w komisji. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań. Ogłaszam 5-minutową przerwę.

Wznawiam obrady. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składzie osobowym komisji sejmowej, druk nr 3187. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 3187, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego w celu rozpatrzenia. Głosujemy. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy z druku nr 3163, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję, że Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej w celu rozpatrzenia. Proponuję, na podstawie art. 39 ust. 3 regulaminu Sejmu, aby komisja przedstawiła sprawozdanie w terminie umożliwiającym rozpatrzenie go na bieżącym posiedzeniu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął.

Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3116 i 3156) Proszę panią poseł Barbarę Dziuk o przedstawienie sprawozdania komisji. A państwa posłów proszę albo o wysłuchanie pani poseł Barbary Dziuk, albo o opuszczenie sali plenarnej, jeżeli nie chcą państwo uczestniczyć w omawianiu tego punktu, i toczenie rozmów w kuluarach. Proszę bardzo, pani poseł. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Niniejszym pragnę przedstawić sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3156. Na wstępie chciałabym krótko zasygnalizować doniosłość i wagę tego projektu.

Komisja Europejska wskazała na brak prawidłowej transpozycji art. 14 ust. 1 dyrektywy o zezwoleniach w zakresie obowiązku przeprowadzenia konsultacji planowanych zmian rezerwacji częstotliwości oraz podniosła zastrzeżenia co do przepisów regulujących przebieg aukcji i przetargu. Wątpliwości dotyczą w szczególności niewiążącego charakteru ofert składanych w trakcie aukcji, braku konsekwencji finansowych wycofania się z rezerwacji czy zbyt niskiej wysokości wadium.

Zasadniczym celem nowelizacji jest zatem przede wszystkim usprawnienie przepisów regulujących postępowanie selekcyjne na rezerwację częstotliwości, a w konsekwencji uniknięcie nałożenia na Polskę bardzo wysokich kar grożących za dalsze utrzymanie w mocy nieprawidłowo transponowanych do polskiego prawa przepisów. Oczywiście projekt wprowadza również kilka istotnych zmian, aby dobro rzadkie, jakim są częstotliwości radiowe, było w Polsce rozdysponowane i wykorzystywane maksymalnie efektywnie. Wśród niezwykle potrzebnych narzędzi i mechanizmów wprowadzanych projektem, umożliwiających efektywne gospodarowanie częstotliwościami w Polsce, należy wymienić chociażby możliwość określenia harmonogramu rozdysponowania poszczególnych częstotliwości, możliwość przeprowadzenia postępowania selekcyjnego na częstotliwości zajęte, tak aby od razu w dniu ich zwolnienia nowy podmiot mógł zacząć je wykorzystywać, czy możliwość przeprowadzenia przez prezesa UKE zamiany wykorzystania przez podmiot częstotliwości na inne częstotliwości o analogicznych właściwościach. Przewidziane zatem w projekcie kompleksowe propozycje służyć będą uporządkowaniu widma w danym paśmie i pozwolą np. na dokonanie koniecznych zmian związanych ze zmianą przeznaczenia pasma 700 MHz na potrzeby usług bezprzewodowych czy też z przydzieleniem częstotliwości na potrzeby sieci 5G.

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, do której niniejszy projekt został skierowany w celu rozpatrzenia, zajęła się nim na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. Komisja wnikliwie rozpatrzyła projekt ustawy, przyjmując kilkanaście poprawek techniczno-legislacyjnych zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne. Komisja przyjęła również jedną poprawkę porządkującą, zgłoszoną przez Biuro Legislacyjne, dotyczącą przepisu przejściowego dotyczącego terminu na rozpatrzenie wniosku o wpis urządzenia do rejestru urządzeń radiowych używanych bez pozwolenia. Wysoka Izbo! Mając na uwadze kluczowe znaczenie projektu dla dalszego rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz nowych technologii, komisja rekomenduje przyjęcie sprawozdania zgodnie z przedłożeniem. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. O zabranie głosu w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość poproszę pana posła Krzysztofa Kubowa. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu co do rządowego projektu ustawy o zmianie Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3116. To niezwykle istotny projekt ustawy, ponieważ rozwijająca się telekomunikacja jest jednym z podstawowych filarów dobrze rozwijającej się gospodarki. Prawo telekomunikacyjne dotyczy przepisów z zakresu gospodarowania częstotliwościami, urządzeń radiowych i opłat za częstotliwość. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Zmiany są związane również z koniecznością zwiększenia efektywności gospodarowania widmem radiowym, a w szczególności zmierzają do zapewnienia wzrostu zainteresowania wdrażaniem na rynku telekomunikacyjnym nowych technologii. Jedną z ważniejszych zmian, które zaproponowano, są przepisy dające możliwość zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz czy też usprawnienia postępowania związanego z rezerwacją częstotliwości. Nowelizacja umożliwia ministrowi cyfryzacji określenie harmonogramu rozdysponowania niektórych zasobów częstotliwości, tak aby można było realizować politykę państwa związaną z gospodarką częstotliwościami. Jednocześnie w nowelizacji ustawy zaproponowano modyfikację zasad przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, w tym w szczególności wprowadzenie dodatkowego warunku odmowy dokonania przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej takiego przedłużenia, oraz umożliwienie prezesowi UKE ogłoszenia z własnej inicjatywy przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości nie tylko w przypadku posiadania wiedzy o zainteresowaniu zasobami częstotliwości, które są już dostępne. Umożliwiono także prezesowi UKE, w drodze decyzji, zmianę przydzielonych rezerwacji częstotliwości w celu zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości. Wysoka Izbo! Nowelizacja ustawy idzie w dobrym, oczekiwanym kierunku. Proponowane rozwiązania mają służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu, do realizacji czego są niezbędne zmiany w przepisach prawa.

O zabranie głosu w imieniu klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska proszę pana posła Arkadiusza Marchewkę. Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o zakres projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne, jest to oczywiście wiele spraw dotyczących kwestii merytorycznych, ale na ostatnim posiedzeniu komisji cyfryzacji mówiliśmy o bardzo szczegółowych sprawach, dlatego nie chciałbym już po raz kolejny mówić o tym, jakie jest główne założenie ustawy, z czym to jest związane, tylko chcę mówić o sprawach, które wzbudzają pewne kontrowersje, przy których pojawiają się znaki zapytania. Chcielibyśmy, aby te sprawy zostały nieco inaczej sformułowane, zgodnie z tym, co przedstawia strona społeczna. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że po tym szczegółowym przedstawieniu ustawy Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska przygotował cztery poprawki w czterech istotnych kwestiach, które pojawiały się w czasie konsultacji społecznych. Chciałbym je teraz przedstawić. Mianowicie, pierwsza sprawa, w projekcie ustawy zawarto przepisy, które dają możliwość określania w drodze rozporządzenia harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości. Takie kompetencje otrzyma według tego projektu minister cyfryzacji. To spotkało się z dużym sprzeciwem strony społecznej, przede wszystkim Urzędu Komunikacji Elektronicznej, gdzie nazwane to zostało podczas posiedzenia komisji wrzutką do Prawa telekomunikacyjnego.

Przypomnę tylko, że istnieje oczywiście w obowiązującym prawie i w tej dyrektywie konieczność zapewniania niezależności organów regulacyjnych, a tym bardziej warto zwrócić uwagę, że w tym projekcie nawet nie ma obowiązku współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, więc ministerstwo rzeczywiście chciałoby te kompetencje przejąć, co naszym zdaniem nie powinno mieć miejsca, dlatego proponujemy skreślenie tego punktu. Druga poprawka również odpowiada na wnioski, które zostały przedstawione w konsultacjach społecznych.

A więc to jest druga kwestia, druga poprawka. Trzecia poprawka stanowi uzupełnienie obowiązującego przepisu dotyczącego wpisu do rejestru urządzeń poprzez wskazanie, że o wpis do rejestru może wnioskować nie tylko właściciel rezerwacji, ale także podmiot przez niego upoważniony.

To jest trzecia poprawka. Może powiem inaczej.

Dlatego należy zaznaczyć, że w warunkach tego obecnego zagęszczenia urządzeń radiowych zadania monitoringu czy też sprawdzania i mierzenia źródeł emisji mogą być skutecznie realizowane z wykorzystaniem mobilnych stacji pomiarowych, dlatego uważamy, [[Dzwonek]] że ten przepis nie powinien zostać zawarty. W związku z tym i z opinią, którą przedstawiłem, w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska składam na ręce pani marszałek cztery poprawki do tego projektu ustawy. Zapraszam pana posła Macieja Masłowskiego, który przedstawi stanowisko w imieniu klubu Kukiz’15. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Proszę państwa, dyskutujemy oczywiście o ważnym projekcie. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące projektu ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Natomiast ciężko jest nam głosować, ciężko nam jest poprzeć tę ustawę, jeżeli mamy tyle niejasności, o których zresztą wspomniał przed chwilą mój kolega, pan poseł Marchewka, i szkoda byłoby to powielać w tym miejscu. Natomiast ja jeszcze dopuszczam to, że są pewne nieprawidłowości, ale Wysoka Izba, cały Sejm jest po to, aby te wątpliwości ewentualne rozwiać. No i niestety na to nie było szans, dlatego że było tragiczne - bo inaczej tego nie nazwę - prowadzenie ostatniego posiedzenia komisji przez pana wiceprzewodniczącego, który zabierał głos pani dyrektor z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, która chciała wyjaśnić, która twierdziła, że potrzeba jej jeszcze 2 minut, żeby nam te wszystkie kwestie wyjaśnić. Natomiast on powiedział, że nie, cytuję: bardzo długo pani mówi, dziękuję za pani wypowiedź. Dlatego będziemy się przyglądać, czy poprzecie państwo poprawki. Podejrzewam, że nie. Dlatego od razu informuję: nie liczcie na to, że my przyłożymy rękę do takiego stanowienia prawa, jakie wy próbujecie wprowadzić. Dziękuję panu posłowi. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W czasie pierwszego czytania nasz klub zajął stanowisko, które przedstawiłem, omawiając rządowy projekt Prawo telekomunikacyjne, dotyczące kontynuowania prac nad tymi zapisami. Wyraziłem nadzieję, że będziemy mogli uzyskać informację, wyjaśnić pewne kwestie i wątpliwości. Jak wspominali już moi przedmówcy, troszeczkę rzeczywistość i praca w komisji rozminęły się z naszymi oczekiwaniami.

Wielokrotnie już przekonaliśmy się, że życie niesie inne rozwiązania.

Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. W imieniu klubu Nowoczesna głos zabierze pan poseł Mirosław Suchoń. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Nowoczesna w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw po przedstawieniu sprawozdania komisji, druki nr 3116 i 3156. Wysoka Izbo! Przedmiotowy projekt ustawy ma na celu dostosowanie naszego prawa do dyrektyw europejskich.

Jednocześnie rząd proponuje w tej nowelizacji pewne przepisy umożliwiające wprowadzenie ładu w gospodarce częstotliwościami. Muszę powiedzieć, że projekt ustawy jest oczywiście niezwykle ważny, ponieważ w tle tego projektu mamy do czynienia z rozwojem sieci inteligentnych, sieci w standardzie 5G. Generalnie chodzi o zagwarantowanie poprawnego wdrożenia technologii przyszłości.

W związku z tym otoczenie prawne, które Wysoka Izba tworzy, również musi być najwyższej jakości. Z tego punktu widzenia muszę powiedzieć, że nasze wątpliwości, które zgłaszaliśmy podczas pierwszego czytania, nie zostały rozwiane podczas posiedzenia komisji.

O co chodzi?

Zgadzamy się z argumentacją Urzędu Komunikacji Elektronicznej, że pozostawienie w urzędzie, przypisanie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej tych kompetencji jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. Muszę powiedzieć, że podczas posiedzenia komisji rząd nie wyjaśnił, dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję dotyczącą rozwiązania prawnego. Zgadzam się również ze stroną społeczną, jeżeli chodzi o kwestię konkurencyjności. Mamy do czynienia z projektem ustawy, który w praktyce likwiduje opłatę za wzrost wartości częstotliwości w przypadku zmiany rezerwacji.

Dlatego zwracam się do pani minister, żeby jednak podjąć ten temat.

To nie jest właściwe podejście do tworzenia odpowiedniego środowiska prawnego dla funkcjonowania gospodarki.

Jeżeli państwo teraz wprowadzą taki zakaz, to okaże się, że Polacy nie będą mogli korzystać z tych prędkości w odpowiednim wymiarze, co oczywiście utrudni funkcjonowanie w gospodarce.

Bardzo proszę, panie pośle. Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Szanowna Pani Minister! Jeśli chodzi o technologię 5G, to ja przyznaję, że nie znam się na tym. Nie muszę się na wszystkim znać, tak jak niektórzy, którzy uważają, że na wszystkim się znają. 13 stycznia złożyłem interpelację w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego. Przywołałem tutaj stanowisko Rady Europy z 2011 r., rezolucję 1815, w której czytamy: Należy podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu zmniejszenia ekspozycji na pole elektromagnetyczne, głównie częstotliwości radiowe emitowane przez telefony komórkowe, szczególnie w przypadku dzieci, młodych ludzi najbardziej narażonych na zachorowanie na nowotwory mózgu. W 2016 r. Europejska Akademia EUROPAEM stwierdziła: Istnieją silne dowody na to, że długoterminowa ekspozycja na pole elektromagnetyczne może powodować wzrost zachorowań na nowotwory, alzheimera i bezpłodność.

Chodziło o to, aby pan premier Mateusz Morawiecki zlecił badania w postaci ekspertyz naukowych na temat wprowadzenia na terenie państwa polskiego technologii 5G. Czy pan premier Mateusz Morawiecki zapoznał się oraz poinformował prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr. prawa Dudę o planowanym wdrożeniu w Polsce w życie technologii 5G oraz o wpływie tej technologii na życie i zdrowie Polek i Polaków, mając na uwadze przytoczony przeze mnie cytat ze stanowiska Rady Europy w 2011 r. wyrażonego w rezolucji 1815? W trzecim pytaniu pytam pana premiera Mateusza Morawieckiego: Czy premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej pan Mateusz Morawiecki zapoznał się w całości z apelem z 13 września 2017 r. ponad 180 naukowców i lekarzy z 36 krajów, którzy domagali się zawieszenia technologii 5G w Europie, oraz jakie jest stanowisko premiera w tej sprawie?

Nie znam się na tym, więc poddałem to w wątpliwość.

Ręce opadają. Dziękuję uprzejmie. Zamykam więc listę. Rozpoczynamy od pytania pana posła Pawła Bańkowskiego, Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam pytanie, czy prawdą jest, jak wynika to z opinii Biura Analiz Sejmowych, że projekt tej ustawy bardzo ogranicza pewność prawną w zakresie wykonywania uprawnień do częstotliwości poprzez wprowadzenie nowych tytułów do cofania, zmiany, odmowy udzielenia rezerwacji na kolejny okres oraz możliwości przymusowej zamiany zasobów częstotliwości przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej? Czy prawdą jest, że zmiany te mogą ograniczyć skłonność przedsiębiorców do podejmowania inwestycji w infrastrukturę sieci bezprzewodowych? I czy prawdą jest, że sposób określania niektórych uprawnień prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do ustalania warunków udziału w postępowaniach selekcyjnych narusza unijne wymagania dotyczące obiektywnego i jawnego charakteru kryteriów rozdziału uprawnień? Dziękuję bardzo. Zapraszam pana posła Arkadiusza Marchewkę, Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, do zadania kolejnego pytania. Pani Marszałek! Pani Minister! Do 2020 r. tzw. ruch w Internecie będzie trzydziestokrotnie większy niż w 2010 r. i prognozy wskazują, że do 2022 r. generalnie do Internetu rzeczy będzie podłączonych na świecie mniej więcej 20 mld urządzeń. To znaczy, że będziemy musieli przygotowywać nowe rozwiązania, operatorzy będą musieli wdrażać nowe technologie, które będą odpowiadać na te potrzeby, które pojawią się właśnie z wprowadzeniem Internetu rzeczy. Dlatego chciałbym zapytać panią minister o wprowadzenie planu na rzecz rozwoju 5G. Do połowy ubiegłego roku Polska, według propozycji unijnych, miała taki plan przyjąć. Tak się nie stało. Po drugie, jak będzie wyglądał model budowy sieci piątej generacji?

Uważam, że do tej pory te działania, które miały miejsce, kiedy prywatni operatorzy w ramach konkurencji budowali własne sieci, były dobrym rozwiązaniem. Czy w takim razie państwo chce w tym uczestniczyć i czy to jest w ogóle dobre wyjście? Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Wysoka Izbo! planu nie ma, chociaż miał być już rok temu, bo oczywiście musi być. Ta ustawa. Zresztą suchej nitki nie pozostawił wasz urząd, Urząd Komunikacji Elektronicznej, na tych zapisach, które eliminują możliwość działania na rzecz rynku, konkurencyjności i interesu obywateli, czyli niższych cen. Czy aukcja na pasmo, które stworzyło możliwość uzyskania szybkiego Internetu, była błędem? Nie, była dla wszystkich użytkowników korzystna, ceny są niższe, dostępność jest większa, co więcej, wpływy do budżetu są ogromne. Ale czy wklucza możliwość powstania monopolu telekomunikacyjnego na paśmie 700? Oczywiście nie wyklucza, nie może wykluczyć. Pytanie brzmi: Jaka kancelaria pisała takie podpowiedzi?

Dziękuję. Wysoka Izbo! Chciałbym po raz kolejny zapytać: Jak przedłożony projekt pozwala chronić małe podmioty, zwłaszcza operujące na rynku radiowym, w rywalizacji o częstotliwość z dużymi koncernami? Czy projektowane przepisy odnoszące się do opłaty za wnioski o rezerwację częstotliwości mogą jednocześnie spełnić rolę w zakresie ograniczenia składania wniosków przez dysponujące poważnymi środkami finansowymi koncerny bez ryzyka ograniczania takiej możliwości np. podmiotom rozpoczynającym działalność? Dziękuję. Zapraszam pana posła Antoniego Mężydłę, który zada kolejne pytanie w tym punkcie posiedzenia Sejmu. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Pani Minister! Myślę, że wada tej ustawy i te wszystkie wady, które zostały tu wytknięte, wynikają z jednego - z tego, że rząd nie zrealizował strategii rozwoju 5G. Gdyby była cała strategia 5G, to nie trzeba by było sobie zostawiać tych nadzwyczajnych narzędzi, które rząd chce mieć, czyli wyręczyć, jeśli chodzi o przydział częstotliwości, Urząd Regulacji Energetyki, ze względu na to, że rząd może prawem, legislacją, legislacyjnie zmusić regulatora do tego, żeby wykonał dokładnie to, czego chce minister. Tu przykładem jest pan minister Halicki. Ja uważam, że. Ja nie cieszę się z tych pieniędzy, wolałbym, żebyśmy mieli szerokie pasmo. Natomiast, pani minister, wczoraj dowiedziałem się, że akurat premier jest zwolennikiem 5G nie z tego powodu, dla którego ja walczyłem [[Dzwonek]] - chodzi o LTE Advanced - tylko z tego powodu, że się boi populistów, którzy mówią o działaniu pola elektromagnetycznego, i chce ustawić jak najmniej stacji bazowych telefonii komórkowej. Z tym się nie zgadzam. Gdybym nie przeczytał wczorajszego artykułu, to myślałbym, że właśnie z tego powodu, że chce stworzyć.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Chcę zapytać o koszty tego przedsięwzięcia, które dotyczy przeniesienia telewizji naziemnych na nowe pasma częstotliwości poniżej 700 MHz. Mam jednak wątpliwości, czy i w jaki sposób zabezpieczyć nadawców telewizyjnych, w tym telewizję publiczną, Telewizję Trwam oraz wszystkie inne działające na naziemnych multipleksach, przed przerzuceniem przez Emitela na nich jednak tych kosztów w umowach cywilnoprawnych, które są zawierane na zasadzie wolnego rynku.

W takim razie czy nie lepiej, żeby to [[Dzwonek]] budżet państwa pokrywał te koszty? O odpowiedź na to oraz na wcześniejsze pytania poproszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji panią Wandę Buk. Bardzo proszę. Szanowni Państwo Posłowie! Szanowni Panowie Posłowie! Przede wszystkim chciałabym zacząć od tematu harmonogramu, który już wielokrotnie był podnoszony i w komisji, i w trakcie dzisiejszego posiedzenia. Odnosiłam się już wielokrotnie do zarzutów, które państwo stawialiście, odnosiłam się do nich merytorycznie, i mam wrażenie, że ani razu nie zostały moje odpowiedzi usłyszane przez państwa i wzięte pod uwagę, co dla mnie jest jednoznacznym sygnałem, że państwa uwagi nie mają charakteru merytorycznego, mają jedynie charakter politycznej tromtadracji i tylko i wyłącznie po to są cały czas podnoszone. Przepisy dotyczące harmonogramu, które wprowadziliśmy, które zaproponowaliśmy w zmianie Prawa telekomunikacyjnego, mają przede wszystkim na celu domknięcie systemu, jaki dzisiaj funkcjonuje w Polsce.

Natomiast rząd nie dysponuje żadnymi narzędziami, które pozwoliłyby mu tych zobowiązań dotrzymać. Tymi narzędziami dysponuje prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zaproponowany harmonogram ma na celu tylko i wyłącznie domknięcie tego systemu i doprowadzenie do tego, aby rząd mógł skutecznie egzekwować od regulatora wypełnianie zobowiązań unijnych. Chciałam tutaj podkreślić jeszcze fakt, że nie jest to żaden wyłom.

Wprowadzenie harmonogramu w żaden sposób nie wpływa na kompetencje regulatora rynku telekomunikacyjnego w zakresie rozdysponowywania zakresów częstotliwości i jego wyłączną właściwość w tym obszarze.

Dodatkowo w samym projekcie nowelizacji rozszerza się jego kompetencje np. o możliwość ogłoszenia postępowania selekcyjnego w sprawie zasobów, które będą dostępne jedynie w przyszłości. Podkreślam: harmonogram nie godzi w zasadę niezależności regulatora, nie ma charakteru instruktażowego, a minister przy jego ustalaniu jest ograniczony przepisami prawa - wydaje harmonogram w formie rozporządzenia, rozporządzenie jest konsultowane, musi być zgodne z przepisami radiokomunikacyjnymi, z polityką i koordynacją widma radiowego określoną w wieloletnich programach unijnych.

Weryfikowaliśmy propozycje tych zapisów, konsultowaliśmy je z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, konsultowaliśmy je również na roboczo z Komisją Europejską. Tutaj tego typu wątpliwości nie ma. I ja już to państwu co najmniej trzykrotnie mówiłam.

I to jest tak naprawdę najważniejsza informacja dla rynku. Właśnie ta ustawa daje nam narzędzia do tego, żeby pokazać, jak i kiedy planujemy wdrożyć tę nową technologię. Przechodzę do pozostałych pytań.

Chciałabym zwrócić uwagę, że Polski rynek telekomunikacyjny jest rynkiem, który jest jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków w Europie. Mamy czterech operatorów mobilnych, mamy jedne z najniższych cen w Europie, natomiast jest to oczywiście działalność bardzo wymagająca, bardzo kosztowna i nie jest to działalność dla małych i średnich przedsiębiorców.

Dziękuję. Po tym wystąpieniu zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Informacja rządu dotycząca wątpliwości pojawiających się wokół śledztwa dotyczącego zabójstwa prezydenta Gdańska pana Pawła Adamowicza oraz funkcjonowania systemu więziennictwa i wymiaru sprawiedliwości. Proszę pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o przedstawienie informacji.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jako że czas niniejszego spotkania, w trakcie którego mam przedstawić państwu szereg informacji, które są istotne zarówno dla opinii publicznej, jak i dla państwa, jest ograniczony, pozwólcie państwo, że skoncentruję się w tym momencie na wyeksponowaniu tych faktów, które wydają się w tym wypadku kluczowe. By przyspieszyć tę relację i by była ona możliwie obfita w fakty, skoncentruję się na odczytaniu dokumentu, gdyż taka forma relacji wydaje się szybsza niż sprawozdanie ustne. Wówczas formuła mojej odpowiedzi będzie inna.

Otóż osoba ta została skazana wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 29 maja 2014 r. na karę łączną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za cztery przestępstwa popełnione w okresie od 8 maja 2013 r. do 12 czerwca 2013 r., które były zakwalifikowane jako rozbój w trybie podstawowym i w trybie kwalifikowanym w charakterze zbrodni w związku z uszczerbkiem doznanym przez osoby, które pracowały w tych instytucjach finansowych. W jednym przypadku była to filia banku Crédit Agricole, o ile pamiętam. Nie będę państwu opisywał szczegółów zarzutów i późniejszej sentencji sądu, w której przypisuje się odpowiedzialność karną temuż sprawcy za te przestępstwa.

Otóż skazany Stefan W. odbył w całości karę orzeczoną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności wymierzoną wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku. Skazany w izolacji penitencjarnej przebywał od dnia 14 czerwca, kiedy to został doprowadzony do Aresztu Śledczego w Gdańsku.